Wznawiam posiedzenie. Na sekretarza dzisiejszych obrad powołuję pana posła Pawła Rychlika, który prowadzić będzie protokół i listę mówców. Obecnie przystąpimy, proszę państwa, do stwierdzenia kworum, dlatego bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu.

Dziękuję.

Właściwe komisje przedłożyły sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, druk nr 2171. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Pan poseł Braun złożył sprzeciw. W związku ze zgłoszonym sprzeciwem sprawę tę rozstrzygniemy w głosowaniu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za skróceniem terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm propozycję przyjął. Proszę państwa, mogę prosić o powstanie? Dzisiaj mija kolejna bardzo bolesna dla nas, Polaków, rocznica zbrodni katyńskiej.

Bardzo proszę, żebyśmy uczcili chwilą ciszy pamięć o wszystkich tych zamordowanych w bestialski sposób przez Rosjan.

Bardzo dziękuję. Mamy wnioski formalne. Pani Marszałek! Składam wniosek o przerwę i chciałam się zwrócić do Wysokiej Izby, w szczególności do rządzącej części, o refleksję nad tym, co wydarzyło się wczoraj. Państwo polskie ma obowiązek stać na straży godności każdej i każdego z nas. Często powinno też stawać po stronie tych, którzy bronić się nie mogą. To, czego dopuściło się wczoraj ministerstwo obrony, to jest rzecz karygodna. To jest uderzenie w nasze serca i nasze dusze. Publikacja zdjęć zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej, brutalnych, okrutnych zdjęć. To brak szacunku. To zabieranie nam wspomnień o ludziach, których znaliśmy i kochaliśmy, tak jak wszyscy tu siedzimy w tej Izbie. Dla jednych to brat, dla drugich to matka, dla innych to mąż (Dzwonek), ale wszyscy tak samo cierpimy.

Wysoka Izbo! Zwracam się z wnioskiem o odroczenie posiedzenia do czasu pojawienia się na sali pana prezesa NBP Adama Glapińskiego i wyjaśnienia posłom i posłankom destrukcyjnej polityki Narodowego Banku Polskiego (Oklaski), która doprowadziła dzisiaj do totalnej inflacji wynoszącej 10,9%. Rozumiem, że rośnie inflacja i rosną pensje?

Pani poseł, czy pani mnie naprawdę nie słyszy?

Pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo szybko pogarszającą się sytuację w kołach łowieckich.

Szanowni Państwo! Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa.

Panie Premierze! Ten temat jest naprawdę bardzo ważny. Dziękuję, panie pośle.

Wnoszę o przerwę celem zwołania Konwentu Seniorów celem wprowadzenia do harmonogramu dzisiejszego posiedzenia, które nagle okazało się wolne od innych przewidywanych zajęć, debaty o polskiej polityce zagranicznej. Jesteśmy za półmetkiem tej kadencji i nie było takiej debaty. Nie było jej wtedy, kiedy państwo wpychaliście Aleksandra Łukaszenkę głębiej w objęcia Włodzimierza Putina. Nie było debaty o sprawach polityki zagranicznej, kiedy wprowadzaliście Polskę w charakterze strony wojującej w tę wojnę, która trwa. Zdaje mi się, że pan prezydent nie przedstawił zarządzenia o stanie wojennym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękuję. Bardzo proszę. W związku z tym nie będę poddawać pod głosowanie wniosku o przerwę. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Chciałem inaczej ten wniosek uzasadnić, ale wobec tego, co się wydarzyło przed chwilą w tej Izbie, nie sposób nie odnieść się do tych pseudoprzeprosin, które wygłosił pan Antoni Macierewicz. Chcę na ręce pani Barbary Nowackiej i wszystkich rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej złożyć przeprosiny, powiedzieć, że my przepraszamy naprawdę i nam jest naprawdę bardzo przykro wobec tego, co się stało [[Głos z sali: W imieniu SB.]] ...i naprawdę uważamy, że do takich rzeczy nigdy nie powinno dochodzić. Pamięć ludzi, którzy zginęli w tej katastrofie, jest święta i tę świętość naruszono, a Antoni Macierewicz, który tu przed chwilą wyszedł, nie potrafi nawet grzecznie powiedzieć: przepraszam. Jest mi wstyd, panie Macierewicz, za pana. Ponieważ został zgłoszony wniosek formalny o odroczenie posiedzenia, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 32. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (druki nr 2170 i 2171) Proszę pana posła Pawła Hreniaka o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Premierzy! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, druk nr 2170. Marszałek Sejmu zgodnie z regulaminem Sejmu skierowała uchwałę Senatu w powyższej sprawie do połączonych komisji w celu jej rozpatrzenia. Połączone komisje na posiedzeniu 13 kwietnia uchwałę rozpatrzyły i wnoszą, aby Wysoki Sejm raczył poprawki od 2. do 6., 9., 11., od 14. do 16., od 18. do 20., 23., 24. i od 26. do 30. przyjąć, a poprawki 1., 7., 8., 10., 12., 13., 17., 21., 22. i 25. odrzucić. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o jej przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę Senatu przyjął. Komisje wnoszą o ich przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki Senatu przyjął. Kto jest za odrzuceniem 4. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę Senatu przyjął. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 7. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę Senatu. Kto jest za odrzuceniem 8. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę Senatu odrzucił. Kto jest za odrzuceniem 9. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę Senatu przyjął. Kto jest za odrzuceniem 10. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę Senatu. Kto jest za odrzuceniem 11. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przeczytam numery poprawek, nie numery głosowań.

Bo na naszej tablicy jest.

Kto jest za odrzuceniem 12. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Kto jest za odrzuceniem 13. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę Senatu odrzucił. Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Kto jest za odrzuceniem 16. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Panie pośle, czy może pan te komentarze zostawić dla siebie? To bardzo proszę, żeby pan je zostawił dla siebie.

10 - za, 447 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm poprawkę Senatu przyjął.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić się do Wysokiej Izby o to, aby odrzucić tę poprawkę Senatu. Polska jest liderem, jeśli chodzi o wprowadzanie sankcji na rosyjskie węglowodory, na rosyjskie surowce. Wyprzedziliśmy wszelkie decyzje, które powinny zapadać na forum Unii Europejskiej. Dlatego, mimo że jesteśmy za sankcjami, uważamy, że ta poprawka jest poprawką złą i szkodliwą.

Mianowicie mówimy o gazie, który jest używany do napędzania samochodów.

Produkcja krajowa to 530 tys. t. Pokrywa to ok. 20% zapotrzebowania na ten surowiec w Polsce.

65% importu pochodzi z Rosji. Tak jak deklarował publicznie pan premier Mateusz Morawiecki, do końca tego roku Polska przestanie importować jakiekolwiek surowce energetyczne z Rosji.

Pozbawianie Polaków w tym czasie możliwości tankowania tańszego paliwa jest czymś okrutnym, szczególnie że dotyczy to Polaków mniej zamożnych.

Chcecie im powiedzieć, że dzisiaj tego paliwa ich pozbawicie. I wreszcie ta cała rzesza osób, które używają butli na gaz.

W tej chwili odchodzimy od węgla, a w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, do końca roku, tak jak zadeklarowaliśmy. odejdziemy również od importu pozostałych surowców energetycznych: ropy i gazu, w tym również gazu LPG. Prosimy bardzo państwa, żebyście nam w realizacji tego zadania nie przeszkadzali, nie próbowali nam pomagać w ten sposób, że nam przeszkadzacie. Nie możemy dłużej wspierać pieniędzmi rosyjskiej machiny wojennej i nie będziemy tego robić. Zachęcam państwa z Platformy Obywatelskiej, z Lewicy, abyście zaapelowali do swoich kolegów z Europejskiej Partii Ludowej, którzy dzisiaj są politykami, którzy rządzą w wielu krajach, abyście zaapelowali do swoich kolegów w rządzie niemieckim, żeby poszli naszą drogą, żeby jak najszybciej odchodzili od dostaw gazu i ropy z Rosji, żeby przestali finansować machinę wojenną Putina. Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Jesteśmy przy głosowaniach, a nie przy debacie. Kto jest za odrzuceniem 17. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

To było wystąpienie zgodnie z regulaminem członka rządu.

Sejm odrzucił poprawkę Senatu. Kto jest za odrzuceniem 18. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

1 - za, przeciw - 454, nikt się nie wstrzymał. Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę Senatu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm przyjął poprawkę Senatu. Kto jest za odrzuceniem 30. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 52. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu. Proszę państwa, pozwólcie jednak, że wszystkim państwu złożę życzenia spokojnych, pogodnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych. Wszystkiego najlepszego dla państwa i dla państwa rodzin.